Wysoka Izbo.

Wprowadzanie pod obrady Wysokiej Izby uchwały jednej, drugiej i trzeciej odwołujących się do skądinąd bardzo ważnych faktów historycznych zakrawa na groteskę, ponieważ okupanci, ani narodowi socjaliści niemieccy, ani międzynarodowi socjaliści sowieccy, nie ważyli się dokonać tego, czegoście wy właśnie dokonali.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za wyrażeniem zgody na zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu w przypadku druków nr 371, 372 i 373, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm propozycję przyjął. Senat podjął uchwały zawierające poprawki do ustaw: - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także: - o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Uchwały Senatu to odpowiednio druki nr 367 i 369. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych uchwał. Proponuję na podstawie art. 54 ust. 8 regulaminu Sejmu rozpatrzenie poprawek zawartych w uchwałach Senatu bez uprzedniego kierowania ich do komisji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, druk nr 374. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 32. porządku dziennego: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie (druk nr 371) Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. W 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd jej ofiarom i bohaterom, poległym żołnierzom i ludności cywilnej. Była to największa i najbardziej brutalna wojna w historii ludzkości. Do jej wybuchu doprowadziły dwa reżimy totalitarne: nazistowskie Niemcy i komunistyczny Związek Sowiecki.

Wojna przyniosła śmierć dziesiątkom milionów ludzi, tragedię Holocaustu, unicestwienie dorobku materialnego i kulturalnego całych narodów oraz eksterminację ich elit. Choć w 1945 r. cały świat cieszył się z pokonania hitlerowskich Niemiec, koniec II wojny światowej nie przyniósł państwom Europy Środkowej i Wschodniej wolności, lecz nowe uzależnienie i komunistyczne zniewolenie. W istocie eliminacja skutków II wojny światowej możliwa była dopiero w momencie wycofania sił zbrojnych Związku Sowieckiego, a następnie Federacji Rosyjskiej z Europy Środkowej i Wschodniej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim Polakom, którzy stali się ofiarami II wojny światowej - żołnierzom, członkom ugrupowań partyzanckich, uczestnikom ruchu oporu, członkom Polskiego Państwa Podziemnego oraz ludności cywilnej. Mając na względzie pamięć o nich, a także dobro ich rodzin i całego państwa polskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku, że siła nie może się opłacać agresorowi i dlatego niezałatwione do dziś, słuszne i zgodne z zasadą sprawiedliwości, roszczenia Polski i Polaków powinny być zaspokojone. Jednocześnie, mając na uwadze ogrom ludzkiego cierpienia i straty materialne poniesione przez narody Europy Środkowej i Wschodniej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednoznacznie sprzeciwia się próbom zakłamywania historii i oskarżania faktycznych ofiar o spowodowanie wybuchu wojny. Rewizjonizm historyczny i manipulowanie faktami stanowią brak szacunku dla pamięci ofiar, budzą również uzasadnione obawy przed kwestionowaniem ładu międzynarodowego opartego na prawie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kieruje wyrazy solidarności do państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym do państw bałtyckich, tj. Estonii, Litwy oraz Łotwy, których parlamenty wielokrotnie zabierały głos w sprawie manipulowania historią. Zwraca również uwagę na Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do przeciwstawienia się próbom rozmywania odpowiedzialności za dramat milionów obywateli Europy i świata. Jedynie pamięć o ofiarach reżimów totalitarnych i szacunek dla prawdy historycznej mogą być fundamentem pokoju w Europie. Proponuję przyjęcie tej uchwały przez aklamację. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 33. porządku dziennego: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w 75. rocznicę utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” (druk nr 372) Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 75. rocznicę utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej 'Warta' Dnia 10 maja 2020 r. przypada 75. rocznica powstania Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej 'Warta', organizacji podziemia niepodległościowego stworzonej na zrębach Poznańskiego Okręgu Armii Krajowej. Warta', założona przez ostatniego komendanta Armii Krajowej w Poznaniu ppłk. Andrzeja Rzewuskiego, ps. 'Hańcza', była apolityczną, konspiracyjną jednostką Wojska Polskiego uznającą zwierzchność Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie. Organizacja formalnie podlegała kierownictwu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Rozbudowywała swoje struktury, zbierała i przekazywała Naczelnemu Wodzowi do Londynu informacje wywiadowcze oraz zwalczała komunistyczną propagandę. Nie podejmując własnych akcji zaczepnych, starano się chronić byłych żołnierzy Armii Krajowej przed prześladowaniami ze strony NKWD i UB. Liczebność organizacji szacuje się na około 5 tys. członków.

W końcowym okresie aktywności 'Warta' była infiltrowana przez agentów UB, co skutkowało, już po formalnym zakończeniu działalności licznymi aresztowaniami. W 75. rocznicę utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej 'Warta' Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wszystkim wielkopolskim żołnierzom drugiej konspiracji, którzy wiernie trwali przy legalnych polskich władzach i walczyli o niepodległość Polski” Proponuję, żebyśmy przyjęli tę uchwałę przez aklamację. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w 75. rocznicę utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 34. porządku dziennego: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii (druk nr 373) Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii. Mając na uwadze, że dokładnie 100 lat temu, 27 maja 1920 r., poseł świeżo powstałej II Rzeczypospolitej Ksawery Orłowski złożył listy uwierzytelniające na ręce ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Brazylii pana Epitácio Pessoa da Silvy, inicjując tym samym proces nawiązywania stosunków dyplomatycznych między obu państwami, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie podkreślić doniosłość tego wydarzenia. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zadowolenie, że owe 100 lat upłynęło pod znakiem konstruktywnej, przyjacielskiej współpracy, i liczy, że kolejne lata i dziesięciolecia będą stanowić okazję do umocnienia się tego trendu, również za sprawą lepszego poznawania się naszych społeczeństw. W dobie ogólnoświatowej pandemii Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża solidarność z narodem brazylijskim, szczególnie tragicznie dotkniętym jej skutkami. Liczymy, że ludzka niezłomność i solidarność międzynarodowa pozwolą nam wszystkim uporać się z zagrożeniem i powrócić na ścieżkę stabilizacji i rozwoju” Bardzo proszę o przyjęcie uchwały przez aklamację. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii. Mamy teraz wnioski formalne. Proszę bardzo, pan poseł Krystian Kamiński, Konfederacja. 1 minuta, panie pośle. Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów, ponieważ dzisiaj debatujemy, będziemy głosować nad czterema umowami międzynarodowymi, w sprawie których nie będzie dzisiaj można zadawać żadnych pytań, a podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji do Spraw Unii Europejskiej nie dostawaliśmy żadnych analiz co do tych umów, czy one się opłacają Polsce, czy nie.

Czy państwo naprawdę sądzą, że powinniśmy w taki sposób procedować nad tym? Moim zdaniem powinniśmy poważnie do tego podchodzić, bo państwo polskie jest suwerennym państwem i powinno samo decydować o tym, co jest dla niego dobre, a co jest złe.

Proszę. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Panie Premierze! Jak wiemy, w Polsce i nie tylko farmaceuci należą do tych, którzy już wiele tygodni temu stanęli na pierwszej linii walki z epidemią koronawirusa, służąc pomocą tym wszystkim, którzy dzisiaj wymagają zaspokojenia potrzeb lekowych. Myślę, że w tym dniu, pani marszałek - dlatego zabieram ten głos - powinniśmy na chwilę odłożyć przedwyborcze emocje, tę bieżącą politykę i skupić się swoimi myślami właśnie na tej grupie bardzo walecznych i pomocnych ludzi, którzy dzisiaj służą naszym rodakom w Polsce, i nie tylko klaskać, tak jak prezes Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, z wdzięczności, ale też uczynić jakiś konkretny gest wobec farmaceutów, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Dlatego chciałbym prosić panią marszałek, aby pochylić się i przekazać do procedowania [[Dzwonek]] projekt „Premia dla bohatera”, wydatnie wychodzący naprzeciw potrzebom. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiciele trzech klubów parlamentarnych: Lewicy, Koalicji Polskiej i Koalicji Obywatelskiej wystąpili do pani marszałek z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o informację prezesa Rady Ministrów w sprawie zakupu za 5 mln zł słynnych środków ochrony osobistej, które jak się okazało, nie spełniały odpowiednich norm. W tej transakcji, tym zakupie dokonanym przez Ministerstwo Zdrowia za 5 mln zł m.in. tych maseczek swoistym pośrednikiem był brat ministra zdrowia pana Szumowskiego.

Każdy kontrahent chciałby być w Polsce tak traktowany, że instytucje publiczne płacą faktury z jednodniowym terminem płatności. Okazuje się, że ministerstwo poddało sprawdzaniu te maseczki dopiero po artykułach prasowych, że coś może być z nimi nie tak, po ponad miesiącu czasu.

Złożyliście państwo dzisiaj po południu te wnioski i oczekujecie, że dzisiaj, kiedy kończymy posiedzenie Sejmu, będzie to rozpatrzone. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby rząd nie odpowiedział na państwa informacje.

Wysoka Izbo!

Na nasze obrady ma czas przyjeżdżać pan premier, pan premier Gliński, pan minister Błaszczak jest prawie zawsze z nami, jest pan minister Kamiński, jest duża część rządu, ale zaginął pan minister Szumowski.

Zgłaszam to dzisiaj, ale też informuję panią marszałek, że wniesiemy na następnym posiedzeniu prośbę o informację pana ministra zdrowia o tym, jak dzisiaj w Polsce rzeczywiście wygląda stan przygotowań do ewentualnej drugiej fali kryzysowej, bo zachorowań nie jest mniej. Mówimy o odmrażaniu gospodarki - i dobrze - ale gdzie poczucie odpowiedzialności za polskie szpitale, służbę zdrowia, pielęgniarki, lekarzy? Nie był to oczywiście wniosek formalny. O głos poprosił pan minister Łukasz Schreiber, członek Rady Ministrów. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję. Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo!

Wysoka Izbo, dzisiaj chyba jasno pokazaliście, że o żaden stan klęski żywiołowej nigdy nie chodziło, że tylko i wyłącznie chodziło o stan klęski sondażowej. Pokazaliście dzisiaj, szanowni państwo, że tak naprawdę wasze słowa o honorze, o szacunku do kobiet są tylko słowami. Pokazujecie tym krzyczeniem, że próbujecie zakrzyczeć rzeczywistość i że debata was w ogóle nie interesuje. Parafrazując słowa Winstona Churchilla, można powiedzieć, że mieliście [[Dzwonek]] do wyboru hańbę albo klęskę.

Pan Łukasz Schreiber jest ministrem - członkiem Rady Ministrów i ma prawo zgodnie z regulaminem zabrać głos. Proszę nie dyskutować ze mną, panie pośle. Bardzo pana proszę. Kto się wstrzymał? Panie pośle, przywołuję pana do porządku. Proszę państwa o to, żebyście nie zabierali głosu w tym trybie. Panie pośle, zabieraliście głos, składaliście wnioski formalne.

Proszę państwa, proszę jedną i drugą stronę o to, żeby zachować spokój, dobrze? Proszę się uspokoić.

jeszcze raz upominam pana. Upominam pana po raz trzeci. Za czwartym razem otrzyma pan ponownie karę. Sam pan o to prosi, panie pośle. Nie, w tej chwili jesteśmy w trakcie głosowania, panie pośle. Ma pan słuchać poleceń marszałka zgodnie z regulaminem.

Sejm wniosek odrzucił.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu w dniu dzisiejszym rekomenduje z tych 87 poprawek 47 poprawek odrzucić, 40 - przyjąć. Wśród tych 40 jest 13 poprawek legislacyjnych, ale również 27 poprawek o charakterze merytorycznym. Z wnioskiem formalnym zgłosił się pan poseł Ryszard Terlecki. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Z wnioskiem formalnym o zmianę trybu głosowania.

Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Głos przeciw. 71 artykułów, każdy o czymś innym. A ze świeczką szukać przepisów, które będą pomagały Polakom w dobie kryzysu polskiej gospodarki. To jest chyba pierwsza w historii cywilizacji europejskiej sytuacja, że gdy Polacy pójdą po bezpłatną poradę prawną, to nie dosyć, że ich dane osobowe będą trafiać do Ministerstwa Sprawiedliwości, ale także informacja, czego dotyczyła porada. Przecież to jest jeden wielki skandal. Pani Marszałek! Pani nam odbiera głos. Pana ministra nie ma, pana ministra finansów od pół roku (Dzwonek) tutaj nie ma.

Dziękuję, pani marszałek. Szanowna Pani Marszałek! My naprawdę chcemy w Izbie normalnie pracować, ale nie może być tak, że pani nadużywa regulaminu i pozwala ministrowi mówić, polemizować z posłem. Formułuję go, ale proszę mi pozwolić. Poseł Konwiński wychodzi i zadaje pytanie w sprawie bulwersującej: 5 mln zł minister Szumowski z własnym bratem za pośrednictwem kolegi trenera, narciarza dał na maski, które były złe. Jak można walczyć z epidemią, wykorzystywać to do wzbogacenia się kolegów? Jak wychodzi minister w imieniu rządu, to powinien powiedzieć: wyjaśnimy tę sprawę, sprawdzamy, służby sprawdzają, nie pozwolimy na to, żeby kraść. A on wychodzi i mówi: poseł Konwiński sobie o czymś porozmawiał.

Panie pośle, jeżeli pan chce przestrzegania regulaminu, musi go pan sam przestrzegać, a pan go notorycznie łamie. Panie Premierze! Wysoka Izbo! Widzicie państwo, jakie te wnioski wzbudzają emocje. Przyznam szczerze, że dzisiaj dyskutowaliśmy przed posiedzeniem Sejmu i dobrze, że się nie założyłem, bo mówię: nie wierzę, że po raz kolejny dojdzie do jakiegokolwiek grupowania. Pamiętam, że dwa posiedzenia wcześniej już tego typu numer również pan marszałek Terlecki zrobił. Jeżeli już nad czymkolwiek mamy głosować, to musimy wiedzieć, nad czym głosujemy. Z całym szacunkiem, panie marszałku, mówienie, że poprawki za są w jednym bloku, a poprawki przeciw - w drugim bloku. Proszę, pani marszałek, o ogłoszenie półgodzinnej przerwy, po to żeby pan wnioskodawca mógł to sformułować i żebyśmy mieli na piśmie, które poprawki chce zblokować. Panie pośle, wniosek o przerwę już był głosowany, natomiast to są poprawki Senatu, a nie Sejmu. Ponieważ został zgłoszony wniosek i głos przeciwny, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem propozycji głosowania łącznego nad poprawkami Senatu zaopiniowanymi pozytywnie oraz nad poprawkami zaopiniowanymi negatywnie przez komisję, zechce nacisnąć przycisk.

Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu.

Wysoka Izbo!

Prosiłbym bardzo, żeby to rzeczywiście rozpisać.

Otrzymaliście państwo sprawozdanie i otrzymaliście państwo. Jeżeli nie 30 minut, to 10 minut przerwy. Niech ktoś nam to wydrukuje, dostarczy tutaj i pokaże. Co to jest za problem? Pragnę poinformować, że druk dotyczący sprawozdania komisji bardzo jasno to określa. Wobec tego każdy wie, nad którą poprawką będzie głosowanie, w którym bloku. Przyjąć, odrzucić - taka jest rekomendacja. Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego. Pani marszałek, pani powiedziała tak: Przeczytam powoli poprawki i wszyscy będą mieli prawo głosować. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przygotowaliśmy się nie z jednej poprawki i nie: przeciw, za. Na posiedzeniu komisji rozmawialiśmy o każdej z tych poprawek, chcieliśmy głosować nad poprawką co do stanowiska: przeciw, za, wstrzymać się. Taka jest rekomendacja, bo tak Lewica uważa. To, co dzisiaj tutaj się stało, to jest utrudnianie wykonywania mandatu posła, uczciwie mówimy. Bo nie chodzi o to, żeby szybko przegłosować, tylko mądrze przegłosować, zrobić prawo, które wszystkim odpowiada, siedzieć 4 godziny - to siedzieć, a nie zrobić to w 20 minut, żeby szybciej pójść do domu. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 367) Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest odrzuceniem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 31. porządku dziennego: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 369) Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

Z poprawką tą łączy się poprawka 3. Proponuję, aby Sejm wyraził zgodę na łączne głosowanie nad poprawkami 1. i 3. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Za - 3, 450 - przeciw, 1 się wstrzymał.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 199. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 199, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. Powracamy do rozpatrzenia punktu 23. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 200. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 200, zechce

Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. Powracamy do rozpatrzenia punktu 24. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 305.

441 było za, 6 - przeciw, 1 się wstrzymał. Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r. Powracamy do rozpatrzenia punktu 25. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 346. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 346, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. Powracamy do rozpatrzenia punktu 29. porządku dziennego: Informacja Rządu w sprawie sytuacji na rynku kredytowym w związku ze skutkami pandemii COVID-19. Wobec propozycji przyjęcia informacji do wiadomości zgłoszono sprzeciw. Pod głosowanie poddam wniosek o przyjęcie informacji do wiadomości. W jakim trybie? Art. 182 ust. 2, panie pośle. Korzystam z tego. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem do wiadomości informacji Rządu w sprawie sytuacji na rynku kredytowym w związku ze skutkami pandemii COVID-19, zechce nacisnąć przycisk.

Pod głosowanie poddałam wniosek o przyjęcie informacji do wiadomości, a w związku z tym, że był zgłoszony sprzeciw, to pytanie brzmiało: Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem... Informacji. Tak jak to wcześniej powiedziałam: Kto jest za przyjęciem informacji do wiadomości. Więc jeszcze raz powtarzam, bo zgłaszają mi posłowie. Ale jeszcze nie zakończyłam głosowania, panie pośle, więc ono cały czas trwa. Złożyliście państwo sprzeciw wobec przyjęcia tej informacji. Proszę państwa, jeszcze raz. Wiem, że jest późno, ale skupcie się państwo.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem do wiadomości informacji rządu w sprawie sytuacji na rynku kredytowym w związku ze skutkami pandemii COVID-19, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest za przyjęciem informacji? - tak było sformułowane pytanie.

Sejm informację przyjął. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 11. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Na tym kończymy 11. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.